Wznawiam obrady. Bardzo proszę państwa posłów o zajmowanie miejsc.

Proszę państwa, wczoraj został zgłoszony wniosek formalny Koalicji Obywatelskiej o przerwanie posiedzenia, w związku z czym ten wniosek formalny przegłosujemy. Dobrze. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Informuję, że wszystkie łącznie głosowane poprawki wynikają z wniosków podmiotów je zgłaszających. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Teraz oczywiście poczekamy, bo państwo wiecie, że musimy dłużej poczekać.

Poproszę o wyniki.

Przechodzimy do rozpatrzenia 3. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przechodzimy do rozpatrzenia 5. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 9. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 15. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. Wyjątkowo wysoka frekwencja. Jak nigdy. Jak nigdy, proszę państwa. Nie pamiętam, kiedy był taki. Kto z pań i panów posłów. Będę czytała wolniej, bo posłowie sygnalizują, żeby czytać wolniej, więc czytam wolniej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 19. i 20., zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 22. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 26. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę przyjął. Przechodzimy do rozpatrzenia 30. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 30. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druków nr 301 i 301-A, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Informuję, że wszystkie łączne głosowania nad poprawkami wynikają z wniosków podmiotów je zgłaszających. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Sejm poprawki odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 2. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 18. poprawki.

Kto się wstrzymał?

Przechodzimy do rozpatrzenia 18. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 267 i 271) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych zawarte w druku nr 271 do uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej. Senat do ustawy budżetowej na 2020 r., uchwalonej przez Sejm, zaproponował 94 poprawki. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 11 marca rozpatrzyła poprawki Senatu i rekomenduje Wysokiej Izbie wszystkie poprawki odrzucić. Wysoka Izbo! Już nie jako poseł sprawozdawca, jako że nie było to przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych, składam wniosek o przeprowadzenie łącznego głosowania nad wszystkimi poprawkami, czyli przyjęcie bądź odrzucenie w łącznym głosowaniu opinii Komisji Finansów Publicznych, biorąc szczególnie pod uwagę tryb głosowania, jaki dzisiaj przebiega, ale też pamiętając o tym, że okoliczności, które były w momencie uchwalania budżetu przez Sejm, również zgłaszanie poprawek przez Senat i również w czasie prac komisji, są już zupełnie innymi okolicznościami, jaki są dzisiaj. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Proponuję zastosowanie w tym przypadku uchwały nr 4 Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie wykładni art. 54 ust. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. głosowanie łączne nad poprawkami Senatu zaopiniowanymi negatywnie. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji głosowania łącznego. Nad poprawkami Senatu nie przeprowadza się dyskusji. Regulamin... Regulamin. Art. 54 ust. 5a. Sejm rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji, chyba że Sejm postanowi inaczej. W tej chwili o tym postanawiamy, pani poseł. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji głosowania łącznego nad poprawkami Senatu zaopiniowanymi negatywnie, zechce nacisnąć przycisk.

Wreszcie jest tak, jak on lubi. Panie pośle, proszę się nie zapominać.

Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął. Komisja wnosi o odrzucenie tych poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 1. do 94., zechce nacisnąć przycisk.

Pani wystąpienia będą na pewno w protokole, pani poseł.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020. Proszę państwa, ponieważ klub Koalicji Obywatelskiej kilkanaście minut temu zgrupował poprawki i dopiero przekazał je do Biura Legislacyjnego. Proszę usiąść. Dostarczył to kilkanaście minut temu. Proszę nie dyskutować ze mną, pani poseł, bardzo panią proszę. W związku z tym ogłaszam przerwę do

Bardzo proszę państwa posłów z Prawa i Sprawiedliwości o spokój. Dobrze?

Wznawiam obrady. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że wszystkie łącznie głosowane poprawki wynikają z wniosków podmiotów je zgłaszających. Z wnioskiem formalnym pani poseł. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny. Na podstawie art. 184 ust. 3 pkt 1 regulaminu Sejmu zgłaszam wniosek o przerwę i proszę o zwołanie Konwentu Seniorów, który jest niezbędny ze względu na tę wrzutkę, która w ostatniej chwili została przez państwa wykonana. Poprawka dotycząca Kodeksu wyborczego, próba zmian Kodeksu wyborczego na kilka miesięcy, na mniej niż 6 miesięcy przed terminem wyborów jest niezgodna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim jest haniebną próbą wykorzystania debaty nad ustawami antykryzysowymi, nad epidemią do majstrowania w Kodeksie wyborczym, do oszukiwania Polek i Polaków. Jesteśmy tutaj zebrani - wszyscy posłowie, wszyscy parlamentarzyści - po to, żeby zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo, miejsca pracy i bezpieczne. warunki przetrwania tego kryzysu. Przystępujemy do głosowania.

nie przeszedł. Drugi wniosek, pana posła Brauna, jest tożsamy, dotyczy tego samego: przerwy i zwołania Konwentu Seniorów.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 4., zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Ja pana dokładnie słyszę. Informuję, że jesteśmy w trakcie głosowania, panie pośle. Tak nie można pracować w Sejmie.

Jeżeli pan się nie uspokoi, poproszę, żeby pan opuścił salę, albo wykluczę pana z obrad. Oczywiście, że mogę pana wykluczyć z obrad zgodnie z regulaminem, więc proszę pana, żeby pan powściągnął swoje emocje i zachowywał się spokojnie na sali, i słuchał poleceń marszałka Sejmu. Bardzo pana proszę. Będzie chciał pan ze mną podyskutować po zakończeniu - zapraszam. A w tej chwili jesteśmy w trakcie głosowania, więc bardzo proszę, żeby się pan zachowywał godnie na tej sali.

Dziękuję.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Przechodzimy do rozpatrzenia 7. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 7., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia poprawek 8a., 9., 16., 17., 18., 20., 28., 45., 46., 52., 55., 58., 59., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 80., 81., 83., 90., 101., 103., 108., 110., 111., 113., 141., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 150., 152., 153., 156., 167., 173., 174., 179., 183. i 185. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Sejm poprawki odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 25., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawki przyjął. Przechodzimy do rozpatrzenia poprawek 40. i 151. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

po tej poprawce, która.

Tak, nie ma. Powiedziałam, że był błąd w scenariuszu i dlatego się to nie znalazło. Dlatego uprzedzam, że za chwileczkę.

Przeczytam, tylko skończymy to głosowanie.

Sejm poprawki przyjął. To jest poprawka klubu parlamentarnego PSL-Kukiz15.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 44., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 48. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 48., zechce nacisnąć przycisk.

Posłowie albo za późno naciskają. Działa, dlatego że mamy tutaj służby informatyczne, które sprawdzają, i działa. Jeżeli komuś się indywidualnie coś nie uda, są telefony.

marszałek. Sejm poprawkę odrzucił. Ja widzę wyniki, panie pośle, naprawdę.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 70., zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Dziękuję.

Sejm poprawkę odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 74. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 74., zechce nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

Głosowało 441 posłów.

Głosujemy.

Proszę państwa, rozpatrujemy w tej chwili, przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 82. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 82., zechce nacisnąć przycisk.

Nie, nie, na pewno nie pozwolę, panie pośle, żeby pan źle przegłosował poprawkę.

Czyli odczytywałam dobrze, u mnie jest dobrze, natomiast tutaj w zestawieniu był błąd. Czyli żebyśmy się nie pomylili, jeszcze raz przeczytam, proszę zerknąć. Wracamy jeszcze raz do tego głosowania. Macie państwo? Tak, dobrze. Przystępujemy do głosowania.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 85. i 94., zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 86. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 86., proszę nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 91., proszę nacisnąć przycisk.

Poprawka nie przeszła. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 92., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Będziemy nad nimi głosować łącznie. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawki odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Przechodzimy do rozpatrzenia 109. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 109., zechce nacisnąć przycisk.

Rozumiem. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 123. i 124. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 122., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Poprawka została odrzucona.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Poprawki zostały odrzucone. Przechodzimy do rozpatrzenia 140. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 140., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 186., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Przechodzimy do rozpatrzenia 187. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 187., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przechodzimy do rozpatrzenia 199. poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 199., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 201., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy głosowanie poprawek. Teraz mamy zgłoszone trzy zgłoszenia przed całością głosowania.

Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jesteśmy w wyjątkowej chwili, jesteśmy po nocnym głosowaniu, ale państwo nie skorzystaliście z wielu rad i dobrych poprawek, które zgłaszaliśmy. Cieszę się, że przyjęliście naszą propozycję, by bezwarunkowo zwolnić z ZUS-u na 3 miesiące, podczas gdy jeszcze niedawno upieraliście się, że ta pomoc nie jest potrzebna. Cieszę się również, że wreszcie wsłuchaliście w nasz głos i zasiłki będą jednak przedłużone dla osób, które opiekują się dziećmi. Ale niestety po raz kolejny podzieliliście Polaków. Zabrakło wam odwagi do tego, by ratować miejsca pracy. Zabrakło wam odwagi do tego, by nie dzielić przedsiębiorców na lepszych i gorszych. Zabrakło wam odwagi wreszcie do tego, by stanąć i przeprosić wszystkich tych, którzy nie będą mogli skorzystać z pomocy państwa. Jestem ciekawy, czy dzisiaj będziecie w stanie wyjść do tego przedsiębiorcy, który nie uzyska od was żadnej pomocy, bo wykluczyliście przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej dziewięciu osób. Czy będziecie w stanie wytłumaczyć pracownikom, dlaczego nie chcieliście potraktować tak samo osoby, która jutro straci pracę w dużej firmie, firmie produkcyjnej, handlowej tylko dlatego, że nie przyjęliście naszych poprawek. I wreszcie, szanowni państwo, niestety nie zgodziliście się na fundamentalną rzecz: 20 mld zł dla polskiej służby zdrowia. To są pieniądze niezbędne do tego, by ratować ludzkie życia. Nie wprowadziliście tych poprawek, bo nie jesteście gotowi na dialog, bo wartości, o których mówicie, są dla was puste. Współpraca, porozumienie, solidarność nic dla was nie znaczy. Dla was najważniejszy jest tylko i wyłącznie interes wyborczy, dlatego tak usilnie bronicie się przed stanem klęski żywiołowej, dlatego nie chcecie Polakom płacić odszkodowań, dlatego nie chcecie, by Polacy mogli starać się o rekompensaty w sytuacji, kiedy państwo zawodzi. Ale my jesteśmy konstruktywną opozycją. Obiecaliśmy naszym wyborcom pomoc. Obiecaliśmy, że będziemy walczyć chociaż o największe poprawki, o których oni mówią. Tutaj nie wszystko się udało. Wiele rzeczy odrzuciliście, ale ponosicie dzisiaj pełną odpowiedzialność za ten pakiet. Ponosicie pełną odpowiedzialność za każde utracone miejsce pracy. Ponosicie pełną odpowiedzialność za każdą krzywdę ludzką, która zostanie wyrządzona przez wasze tchórzostwo. Żałuję, pani marszałek, że nie dotrzymaliście słowa. Żałuję, panie premierze, że nie dotrzymaliście słowa. Żałuję, że nie skorzystaliście z wyciągniętej ręki, dialogu, porozumienia i dobrej pracy. Dziękuję, panie pośle. To jak przyjdzie, to dopuszczę go do głosu. Proszę. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jest bardzo późno, a w zasadzie bardzo wcześnie. Wielu Polaków wstaje właśnie do pracy. Za to, że dziś, tak jak każdego dnia, pomimo epidemii udadzą się do pracy, do przychodni, do szpitala, ale także do sklepu czy na pocztę. Zrobią to pomimo narażania swojego zdrowia, narażania zdrowia swojej rodziny. Zrobią to dlatego, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie, żebyśmy mogli czuć się zaopiekowani. Bardzo serdecznie im dziękuję, bo to dzięki nim państwo pomimo kryzysu, pomimo epidemii nadal działa. Najwyższy czas, żeby to państwo, które powinno im dzisiaj być wdzięczne, doceniło ich. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił wykorzystać kryzys do tego, by zamiast szacunku okazać tym osobom jeszcze więcej pogardy, obcinając pensje, osłabiając prawa pracownicze. Dzisiaj wszyscy pracownicy i pracownice, 16 mln Polek i Polaków, obawiają się o swoje wynagrodzenia. Projekt ustawy zakłada możliwość obniżania wynagrodzeń o nawet połowę. Czy ministerstwo, czy rząd przewiduje, ile osób otrzyma niższe wynagrodzenia? Ile gospodarstw domowych będzie miało niższe przychody? Czy te wszystkie osoby, które wstają dzisiaj do pracy, mogą czuć się bezpiecznie? Czy rząd planuje jakiekolwiek zabezpieczenia na ten czas, kiedy tą pracę stracą? Prawie 3 mln osób na samozatrudnieniu czy umowach cywilnoprawnych znalazło się dziś w sytuacji bez żadnych zabezpieczeń. Kryzys epidemii pokazał dobitnie, dlaczego pracujące osoby na umowach cywilnoprawnych nazywają te umowy śmieciówkami. Te miliony ludzi stają dzisiaj przed ryzykiem utraty pracy i środków do życia. Wręcz przeciwnie - pogłębiają je. Wasze propozycje osłabiają prawa pracowników, nie zabezpieczają sytuacji osób, które pracę stracą. Odrzuciliście poprawkę Lewicy, dzięki której osoby pracujące na śmieciówkach zyskałyby pełnię praw z Kodeksu pracy. Odrzuciliście poprawkę Lewicy, dzięki której zwiększony zostałby zasiłek dla osób bezrobotnych. Zrobiliście to pomimo ze wiecie, że ok 70% przedsiębiorców grozi dziś pracownikom zwolnieniami. Wiecie o tym, że po fali epidemii nadejdzie fala bezrobocia, i nie zrobiliście nic, żeby ludzi, którzy znajdą się pod tą falą, zabezpieczyć przed utonięciem. Ja z uwagą przysłuchiwałam się dzisiejszym wystąpieniom przedstawicieli partii rządzącej. Powtarzaliście państwo słowo „solidarność”, „solidarność” Dlaczego w waszych ustawach tak niewiele jest solidarności państwa z jego własnymi obywatelami? W czasie takiego kryzysu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, musimy być solidarni, ale naprawdę, troszczyć się o siebie nawzajem - jeden o wszystkich i wszyscy o jednego. Z milionami pracowników, którym w oczy zagląda widmo długotrwałego bezrobocia, nie jesteście solidarni. Chcecie państwo zaciskać pasa, ale boicie się zaciskać pasa na brzuchach tłustych kotów. Wolicie zaciskać pasa na najchudszych, najsłabszych, tym, którym najtrudniej jest upomnieć się o swoje prawa. Bardzo proszę.

Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Jesteśmy po 7 godzinach głosowań nad poprawkami do tarczy antykryzysowej, która niestety nie okaże się skuteczna w takim stopniu, w jakim mogłaby się okazać, w jakim oczekują tego polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy, dlatego że nie skupia się na czterech prostych filarach, które mogłyby pozwolić jej działać szybko i skutecznie, a więc nie ulży w kosztach stałych dla przedsiębiorców, ZUS i podatki, nie da prostego, szybkiego dostępu do kapitału obrotowego, nie da szybkich i działających natychmiast dopłat do miejsc pracy i wreszcie nie wstrzyma wejścia nowych podatków. Nowe podatki zapowiedziane, takie jak podatek cukrowy, mają wejść, nic się w tej kwestii nie zmienia. Zamiast tego będziemy mieć 24 nowe procedury urzędnicze, komisje urzędników, komisje rozpatrujące wnioski, przedsiębiorców piszących wnioski. Kancelarie prawne już w tej chwili proponują usługi polegające na tym, że będą doradzać, panie premierze, jak skorzystać z tych rozwiązań, które pański rząd w tej chwili wytwarza, z tych nowych 24 procesów, które będą uruchamiane w administracji. Jest natomiast grupa, która będzie bardzo zadowolona z tego, jaki kształt ma ta tarcza. Pan premier odniósł się do tej grupy w swoim wystąpieniu, w pewien sposób pokazując, jakiego zarzutu się boi. A mianowicie to są banki. Pan premier wywodzi się z banków i banki są tą grupą, która jest szczęśliwa z kształtu tarczy, którą rząd jej nadał. A to z bardzo prostego powodu: w odróżnieniu od różnych innych państw tarcza zaproponowana przez rząd PiS-u w żaden sposób nie uderza w interesy banków. Nie wprowadza żadnego rozwiązania, gdzie banki musiałyby się podzielić czy to funduszami, czy choćby zyskami z przedsiębiorstwami i zwykłymi obywatelami. Wakacje kredytowe, które będą wprowadzane, będą odpłatne. Rząd nic nie zaproponował w tym zakresie. Wszystkie instrumenty, które rząd zaproponował są natomiast zoptymalizowane dla banków, takie jak obniżenie rezerw, takie jak instrumenty płynnościowe, takie jak gwarancje. Zwykli przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć na takie specjalne traktowanie, na jakie będą liczyć koledzy z branży, wśród których pan premier zdobywał doświadczenie i funkcjonował przez lata. Można powiedzieć, że to przypadek, można uznać, że jest to jednak następstwem pewnych koneksji, pewnych powiązań, które dzisiaj sięgają na najwyższe szczyty władz naszego państwa. To nie jest sprawiedliwe, że zwykły przedsiębiorca nie może liczyć na tak preferencyjne traktowanie, na jakie będą liczyć bankowcy. Panie premierze, nie na to czekali polscy przedsiębiorcy. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, panie premierze.

Wysoka Izbo! Dzisiaj rzeczywiście, dzisiaj i wczoraj dyskutowaliśmy o fundamentalnych sprawach, fundamentalnych sprawach dla pracowników, dla przedsiębiorców. Ja rozumiem, że prawidła tutaj i zwyczaje, które w ostatnich latach sprawiły, że opozycja w mniejszym stopniu merytorycznie odnosi się do tego, co my proponujemy, a w większym stopniu są to różnego rodzaju zaczepki, spowodowały, że ta dyskusja w znacznym stopniu nie odnosiła się do tego, co jest meritum tarczy. Ale meritum tarczy ma obronić przede wszystkim pracowników i przedsiębiorców polskich przed bankructwami. I dlatego raz jeszcze apeluję w ślad za tym, o czym mówiłem na samym początku, nie tylko każdy dzień się liczy, każda godzina się liczy. Dlatego bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat najlepiej jeszcze dzisiaj, jak najszybciej, najlepiej żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, ocalić swój dorobek, bardzo często dorobek życia, a w ślad za tym ile miejsc pracy ocalimy. Więc odłóżmy do lamusa te przepychanki czy te zaczepki, te różne zaczepki, które tutaj padały przez ostatnie 7 godzin. Ja się nie gniewam, wybaczam. Nie przejmuję się tym nadmiernie, ale bardzo proszę państwa wszystkich, głosujmy za tą tarczą jak najszybciej, ponieważ ilość ulg, które tutaj ujęliśmy, ilość bezpośrednich dopłat do pracowników, dla przedsiębiorców jest bezprecedensowa. Ta tarcza jest jedną z największych tarcz do PKB zaoferowanych przez wszystkie inne państwa, w porównaniu do wszystkich innych państw. Wiecie doskonale, bo rozumiem, że tutaj, w tej poetyce czy retoryce, która tutaj była rzucana tak troszeczkę jakby bez odpowiedzialności za słowo, bo myślę że wy doskonale wiecie i państwo, którzy przed chwilą mówiliście, też doskonale wiecie, że pomoc dla przedsiębiorców, pomoc dla pracowników idzie nie w miliardy, nie w dziesiątki miliardów, idzie w setki miliardów złotych, idzie w realnych pieniądzach. Wiecie też doskonale, że akurat banki opodatkowała władza Prawa i Sprawiedliwości, bo to my narzuciliśmy podatek bankowy który właśnie zapobiegł nadmiernej eskalacji kredytowej, nadmiernej ekspansji kredytowej, i dzięki temu pozyskujemy rokrocznie 4 mld zł do budżetu.

Ja to wszystko odkładam do lamusa, nie gniewam się na państwa i bardzo proszę wszystkich, żebyście głosowali za tym, ale nade wszystko wierzę w to, że oczywiście ta ustawa będzie przegłosowana, ona jest bardzo ważna. Proszę Senat, proszę pana marszałka Senatu o zwołanie jak najszybciej posiedzenia, bo, raz jeszcze podkreślam, liczy się każda godzina. Przed meteorytem nikt się nie ubezpiecza, przed koronawirusem nikt na świecie się nie ubezpieczył i nikt na świecie się do niego nie przygotowywał. Takie rzeczy, takie epidemie zdarzają się bardzo, bardzo rzadko i nieszczęśliwie ona nam, Polakom również się przydarzyła. Dlatego w odpowiedzialności za państwo polskie, za polskich pracowników proszę bardzo Wysoką Izbę o zgodne głosowanie nad tą tarczą antykryzysową.

Robimy wszystko, żeby zapobiegać utracie miejsc pracy i zapobiegać bankructwom. Bardzo proszę Senat o jak najszybsze głosowanie, jeżeli tylko Wysoka Izba zgodzi się przegłosować tarczę antykryzysową, w co głęboko wierzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie premierze. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druków nr 299 i 299-A, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 8. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.